Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Małgorzatę Golińską i Piotra Olszówkę. Protokół i listę mówców prowadzić będzie poseł Małgorzata Golińska. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa - godz. 11. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Izbę, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o przeniesieniu na następne posiedzenie Sejmu trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu zwracam się do pana marszałka z prośbą o ogłoszenie przerwy, zwołanie Konwentu Seniorów i podjęcie decyzji o zdjęciu z porządku dziennego punktu 20., czyli sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prawo i Sprawiedliwość już nas przyzwyczaiło, że łamie prawo, łamie konstytucję pod osłoną nocy, ale ta buta i arogancja poszły dalej. Dzisiaj chcecie złamać prawo w dzień powszedni. W dzień, w ciągu dnia. Panie Marszałku! Apeluje pan do nas, żeby utrzymać powagę Sejmu. A co można powiedzieć o działaniu pana marszałka dopuszczającego do procedowania ustawy, która nie została przegłosowana w Senacie?

Umiem liczyć, a wam to, zdaje się, źle idzie.

Panie Marszałku! Bardzo proszę naprawdę poważnie podejść do tej sprawy, dlatego że to jest łamanie prawa w biały dzień. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

I jest to wprost zapisane w regulaminie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym się przyłączyć do wniosku o ogłoszenie godzinnej przerwy dla prezesa rady ministrów gabinetu cieni pana Grzegorza Schetyny, tak aby w ciągu 1 godziny zdymisjonował ministra obrony narodowej w gabinecie cieni Tomasza Siemoniaka. w związku z informacjami, jakie uzyskujemy i otrzymujemy w Polsce, związanymi z caracalami. Szanowni Państwo! Gdyby nie obecny minister obrony narodowej, bylibyśmy w bardzo podobnej sytuacji z serwisowaniem sprzętu i mielibyśmy bardzo niekorzystną umowę offsetową. Panie pośle, przepraszam bardzo, to nie jest wniosek formalny, nad którym możemy głosować, ponieważ nie dotyczy on porządku dziennego. Dziękuję panu bardzo. Poseł Jacek Protasiewicz. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę, panie pośle. Bardzo pana proszę. Proszę opuścić mównicę.

Wczoraj była bardzo dobra inicjatywa, przedłożona przez Konwent Seniorów, ażeby Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą 500-lecie reformacji.

Ale panie pośle, wniosek o przerwę już został zgłoszony, tak że bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

Komisje wnoszą o przyjęcie tych poprawek. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Poprawkę Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Sejm poprawki przyjął. W 3. poprawce Senat proponuje dodać przepis przejściowy. Z tą poprawką łączy się poprawka 5. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Kto jest przeciw? Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poseł Magdalena Kochan, klub Platforma Obywatelska.

Sprowadza się do tego, że o rok opóźniamy wejście w życie szkodliwych przepisów. Szkodliwych, bo zabierają średniakom, a nie dodają złotówki biednym. Szkodliwych na tyle, że pracodawcy ze związkowcami we wspólnym - podkreślam: wspólnym - stanowisku nie zostawili na tych przepisach suchej nitki. One w ogóle nie powinny wejść w życie, bo nie dość, że są szkodliwe, to jeszcze zostały podjęte z wadą legislacyjną.

Tracimy szacunek dla legislacji, tracimy szacunek dla prawa. Głos ma poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ci, którzy mogą zapłacić składkę na ZUS, nie zapłacą jej przez następny rok, za to ci Polacy, którzy z całą pewnością tej składki zapłacić nie mogą, bo ich przychody są porównywalne z ryczałtową składką na ZUS, będą nadal dorzynani ekonomicznie przez państwo polskie. Zapowiedział pan w kwietniu ustawę o małym ZUS-ie dla przedsiębiorców, która miała wejść 1 stycznia 2018 r. Kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Kiedy będziemy mieli sytuację, że państwo będzie pobierało daniny od swoich obywateli w takiej wysokości, w jakiej są oni w stanie je zapłacić? Panie i Panowie Posłowie! Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, chcecie przyjąć tę poprawkę z możliwością naruszenia prawa, bo grunt pali się wam pod nogami, bo zrozumieliście, że wdrożenie tych rozwiązań z nowym rokiem nie jest możliwe, bo zrozumieliście, że opozycja, związki zawodowe, przedstawiciele przedsiębiorców, a także przedstawiciele ZUS, gdy mówili, że to złe rozwiązanie, mieli rację. Panie pośle, identycznie brzmi regulamin Sejmu, a mimo to kworum jest liczone na podstawie dokonanych głosowań. Senatorowie opozycji jednoznacznie zgłaszali, że kworum na sali nie było. Naszym zadaniem jako posłów Rzeczypospolitej Polskiej nie jest liczenie senatorów obecnych albo nie na sali w Senacie. Naszym obowiązkiem jest branie pod uwagę, że prawo być może zostało złamane. Możemy zaapelować do pana prezydenta, aby nie podpisywał tej ustawy, ale nie możemy [[Dzwonek]] legitymizować łamania prawa.

Bo przecież ta ustawa w istocie podnosi podatki. Mówiłem to już kilka razy i należy to powtórzyć, i należy to powtarzać Polakom, żeby Polacy byli świadomi, że państwo podnosicie podatki, mimo że mówiliście, że nie będziecie ich podnosić. A pani Kochan odpowiadam, że my już się przyzwyczailiśmy.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Przystępujemy do głosowania.

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw głosowało 419, za - 1. Sejm poprawki przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Senat proponuje inne terminy na wprowadzenie określonych regulacji prawnych oraz aby ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Komisja wnosi o przyjęcie tych poprawek. Pytanie zadaje poseł Janusz Cichoń, klub Platforma Obywatelska. Wysoki Sejmie! Jesteśmy jedynym krajem, który prowadzenie kont VAT w systemie podzielonej płatności split payment powierza, przekazuje bankom. To gigantyczne darmowe pieniądze na ich kontach zamiast na kontach ministra finansów, zamiast na kontach tak naprawdę państwa. Uzasadnieniem takiej poprawki, takiej decyzji był czas niezbędny na wdrażanie, co dzisiaj wyraźnie okazuje się fikcją, bo to jest kolejna zmiana terminu. Chciałbym zapytać, kto jest autorem tego pomysłu, aby to banki prowadziły te rachunki. Kto jest Świętym Mikołajem? Kto daje takie prezenty bankom i SKOK-om z okazji Bożego Narodzenia?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drogi Rządzie! Szanowni Państwo! Ta ustawa. jest ustawą, która walczy z mafiami VAT-owskimi, mafiami, które wyłudzały miliardy złotych z budżetu państwa. do likwidacji karuzel VAT-owskich, ostatecznej likwidacji tych karuzel VAT-owskich. Banki, droga pani. współdziałały z rządem przy tworzeniu tej ustawy. Banki będą mogły.

Proszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 6. oraz od 8. do 10., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 421 posłów. Za głosował 1, przeciw - 420. Sejm poprawki przyjął.

Czy ktoś z państwa chciałby się dopisać do listy? Proszę bardzo. Jak nikt się nie zgłasza, zamykam listę. Jako pierwszy zgłasza się. Jeszcze do oświadczenia, tak? Jako pierwszy głos zabierze poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony.

Ogłaszam 2 minuty przerwy.

Wznawiam obrady. Zapraszam do wygłoszenia oświadczenia pana posła Jana Mosińskiego, klub Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę państwa posłów i członków rządu o wyciszenie rozmów. Wysoka Izbo! W Wilkowicach, niewielkiej miejscowości nieopodal Leszna w Wielkopolsce, grupa pasjonatów postanowiła założyć Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej, które stało się bardzo aktywną organizacją zrzeszającą mieszkańców Wilkowic i ościennych miejscowości. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowic to serce tego stowarzyszenia, które za główny cel przyjęło kultywowanie tradycji wsi wielkopolskiej. Nie tak dawno miałem zaszczyt uczestniczyć w otwarciu Regionalnej Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej. Powstała ona przy wsparciu księdza proboszcza parafii Wilkowice, ks. Macieja, który oddał budynek gospodarczy znajdujący się na terenie probostwa należącego do kościoła pw. św. Marcina. Po kilku miesiącach intensywnych prac udało się zaadaptować pomieszczenie na wspomnianą przed chwilą Regionalną Izbę Kultury i Tradycji Wiejskiej - jak podkreślali członkowie stowarzyszenia, a także zwiedzający - tak bardzo potrzebną, służącą przekazywaniu przyszłym pokoleniom spuścizny po naszych dziadach i pradziadach. Ta regionalna izba służyć będzie przechowywaniu eksponatów nawiązujących do naszej kultury i tradycji. Prezes stowarzyszenia pan Sylwester Przydrożny podkreślał, cytuję: Za pośrednictwem tej izby pragniemy chociażby w części pokazać, jak duży wysiłek fizyczny musieli ponieść chłopi na wsi, aby zabezpieczyć dostatnie życie swym rodzinom, na jakim sprzęcie pracowali, jak przebiegał postęp i rozwój techniki oraz rzemieślników, którzy pracowali na wsi. To oni głównie byli autorami postępu technicznego w rolnictwie. Dzięki kreatywności, pracowitości i dużemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz mieszkańców nie tylko Wilkowic, ale i gminy powstał ten wspaniały obiekt.

Regionalna Izba Kultury i Tradycji Wiejskiej łączy przeszłość z dniem dzisiejszym, a potwierdzeniem tego jest piękny mural zdobiący budynek, autorstwa państwa Magdaleny i Filipa Rozynków. W tym miejscu muszę poruszyć drażliwą kwestię, mianowicie rolę władz gminnych i wójta Lipna, który zamiast wspierać działania stowarzyszenia, wyszukuje różne działania mające za zadanie utrudnić działalność stowarzyszenia. Szanowny panie wójcie, niech pan otworzy szeroko oczy, rozejrzy się dookoła i dojrzy to piękne dzieło, jakim jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej, i ludzi, którzy społecznie działają w obszarze upamiętniania tego wielkiego dzieła, któremu na imię historia wsi polskiej, historia Wilkowic. A jeśli nie chce pan wspierać działań społeczności lokalnej Wilkowic, to niech pan przynajmniej nie przeszkadza. Kilka dni temu w hotelu Bazar Poznański w Poznaniu odbyła się uroczysta gala konkursu „Działania godne uwagi” Goście gali oprócz wysłuchania wspaniałego koncertu fundacji Pro Musica z Leszna mogli także dowiedzieć się o źródłach finansowania działań lokalnych przygotowanych przez pana Piotra Kotlarka z Centrum PISOP. Podczas gali jednym z laureatów konkursu zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej za adaptację budynków gospodarczych na Regionalną Izbę Kultury i Tradycji Wiejskiej.

Szanowni państwo, raz jeszcze szczerze gratuluję, a zarazem deklaruję, że tak samo jak do tej pory jestem do państwa dyspozycji wraz z moją asystent panią Joanną Nawrot, a także asystentami panami Piotrem Paterczykiem i Tomaszem Piątą. Szanowni państwo, do zobaczenia w Wilkowicach.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mieszkańcy wspomnianych gmin niejednokrotnie zwracali mi uwagę na występujące od wielu lat problemy we współpracy sądów i prokuratury w Pszczynie z Policją i organami administracji publicznej w Bielsku-Białej. Częste problemy we współpracy odbijają się na jakości tych działań. W związku z tym faktem bardzo proszę o to, aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i dogłębnie przeanalizować możliwości dotyczące tego problemu, a także rozważyć przekazanie gmin Bestwina i Czechowice-Dziedzice pod zwierzchność prokuratury i sądu w Bielsku-Białej. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz’15. Wysoka Izbo!

Przy tej okazji wszystkim państwu zebranym na sali, ale również tym, którzy będą słuchać tych słów za pośrednictwem mediów elektronicznych, życzę spokojnych, radosnych, zdrowych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście ten czas spędzili w takiej atmosferze, która napełni was pozytywną, dobrą energią. A później szczęśliwego nowego 2018 r. Dziękuję bardzo.

Wysoki Sejmie! Wczoraj Konwent Seniorów wyszedł z bardzo cenną inicjatywą, ażeby 500. rocznicę reformacji uczcić w Izbie przyjęciem specjalnej okolicznościowej uchwały. Takie uchwały często są podejmowane przez tę Izbę z różnych okazji i muszę powiedzieć w bardzo mocnych i twardych słowach, że jest więcej niż wstydem, chyba nawet powiem, że jest hańbą, że przyjmowaliśmy w tej Izbie uchwałę upamiętniającą Narodowe Siły Zbrojne, w tym kontrowersyjne losy Brygady Świętokrzyskiej - była ona przyjmowana w tej Izbie przez aklamację, zaznaczę, bez mojego fizycznego udziału - a zabrakło odwagi, zabrakło woli, ażeby przyjąć bardzo rozsądną, bardzo stonowaną i bardzo wyważoną uchwałę odwołującą się do historycznego wydarzenia, jakim było ogłoszenie tez Lutra 500 lat temu, i jego konsekwencji zarówno dla kultury europejskiej, jak i dla kultury polskiej. Mówiąc krótko, w Sejmie mieliśmy wolę, ażeby uhonorować postaci kontrowersyjne z naszej historii, a zabrakło woli, ażeby oddać hołd tak wielkim Polakom jak Mikołaj Rej, Andrzej Frycz Modrzewski, gen. Józef Sowiński, Juliusz Konstanty Ordon czy choćby Stefan Żeromski, marszałek Piłsudski czy gen. Władysław Anders.

Ale myślenie o Polakach w kategoriach wyłącznie Polak - katolik jest bardzo niebezpieczne i fałszuje prawdziwą polską historię, wypacza polską tradycję. Koronnym argumentem, który usłyszeliśmy ze strony parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wczoraj sprzeciwiali się przyjęciu tej uchwały, było to, iż nie wolno honorować wydarzenia, które doprowadziło do podziału w Kościele.

Tu nie zebrał się ani synod, ani tym bardziej sobór, ażeby rozstrzygał kwestie religijne. Ale nawet jeśli już parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności pani poseł Siarkowska, próbują używać takich argumentów, to odsyłam do bardzo mądrego, bardzo wyważonego listu, który z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra wystosował Ojciec Święty, wówczas Jan Paweł II, do wspólnoty protestanckiej w Europie. Trzeba się wzorować na tym sposobie myślenia i na tej argumentacji, a nie na sposobie myślenia bliższym ksenofobicznej, nacjonalistycznej tradycji Obozu Narodowo-Radykalnego. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że coraz częściej mam wrażenie, że słowa Tuwima, które zawarł w swoim poemacie „Kwiaty polskie”, o tym, że na ulicy rządzą drobnomieszczańscy drobni dranie, już katolicy, tyle że jeszcze nie chrześcijanie, coraz bardziej pasują do aktualnej sytuacji Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie i Panowie!

Chciałbym, żeby w tym zaszczytnym gronie, panie marszałku, pań i panów posłów dzięki elektronicznym mediom ten silny sygnał uznania, szacunku i podziękowania dla Christiaana Barnarda, jego zespołu i wszystkich transplantologów, którzy to dzieło kontynuują, zabrzmiał szczególnie.

Dzisiaj my tak bardzo pomagamy dzieciom i dorosłym, ratując ich w Kosowie, na Ukrainie. Wśród tych, którzy tak pięknie przejęli inicjatywę prof. Barnarda, był prof. Zbigniew Religa, mój mentor, nauczyciel i przyjaciel, który zaszczepił w nas tę ideę ratowania życia, która będzie ponadczasowa, i tak bardzo wspierał mnie, kiedy podjąłem się pierwszych w Polsce transplantacji serca i płuc.

Chcę również z tej okazji temu wybitnemu Polakowi, prof. Relidze, i innym, prof. Mollowi, podziękować. Na koniec refleksja. Zawsze w tej Izbie jestem i byłem zwolennikiem pokoju, pojednania, współpracy.

Panowie! Bardzo dziękuję. Oświadczenie wygłosi pani poseł Małgorzata Chmiel. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zniszczony został Trybunał Konstytucyjny, sądy, teraz przyszedł czas na nasz system emerytalny. Jeszcze obowiązujące przepisy ustawy stanowią, że po przekroczeniu dochodów w stosunku rocznym powyżej trzydziestokrotności średniej pensji, w tym roku wynosi to ok. 127 tys. brutto, co daje wynagrodzenie ok. 6700 zł miesięcznie na rękę, o takich pieniądzach mówimy, od tej sumy nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne. Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając obowiązkowe składki ZUS od wyższych wynagrodzeń dba jedynie o chwilowe zwiększenie wpływów do budżetu, bo obliczyliście państwo, że da to w przyszłym roku zwiększenie wpływów o ok. 5 mld zł. Ale to jest brak odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Każdy odpowiedzialny rząd powinien myśleć przede wszystkim o przyszłości. Te wysokie emerytury, które z tego będą wynikać, ponieważ im wyższe składki, tym oczywiście wyższe emerytury, będą musiały spłacać nasze dzieci. A wy myślicie tylko o przyszłym roku, o roku wyborczym. Żeby utrzymać dom, rodzinę, musi zarabiać często na dwóch etatach, osiągając dochód powyżej tej trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia. Taka osoba również będzie musiała opłacać wyższy ZUS. Oznaczać to będzie dla takiej osoby dużą obniżkę wynagrodzenia. Wejście w życie tej ustawy spowoduje olbrzymią przepaść w wysokości wypłacanych w przyszłości emerytur. Czy będzie nas stać na wypłatę emerytury w wysokości ok. 40 tys. za kilkanaście lat? To nieprzyzwoite, szczególnie gdy weźmiemy od uwagę, że większość emerytur za kilkanaście lat będzie oscylowała wokół 1500 zł miesięcznie. A może państwo z PiS-u planują po prostu ściągnąć teraz od tych ludzi lepiej zarabiających te 5 mld, żeby były na przyszły rok, bo nie macie na pokrycie swoich zobowiązań, a potem ogłosić, że będzie emerytura obywatelska i wszystkim po równo, i chcecie oszukać tych ludzi, którzy teraz będą płacić te wysokie składki emerytalne? Teraz głos ma pani poseł Joanna Fabisiak, klub Platformy Obywatelskiej. Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym Sejm podjął uchwałę wyrażającą uznanie dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ona nie wybrzmiała, przeszła jakoś tak mimochodem, rzekłabym, i chciałabym podkreślić ten fakt, bo to jest 200. rocznica, w październiku były obchody 200. rocznicy utworzenia i istnienia tej niezmiernie ważnej instytucji humanistycznej. Ja wiem, że żyjemy codziennością, żyjemy sprawami bytowymi, sprawami bardzo ważnymi, ale człowiek pozbawiony humanistyki, pozbawiony książki staje się ubogi i w jakiś sposób bardzo biedny. A jest to zakład szczególny.

Był dla Polaków w okresie niewoli takim powiewem wolności, takim miejscem, gdzie można było prowadzić badania, głównie nad literaturą.

To jest wielkie, piękne, nowoczesne wydawnictwo. Prowadzone są badania. Jest ogromna, wspaniała Biblioteka Narodowa. Jest wreszcie Muzeum Pana Tadeusza. Myślę, że warto, aby każdy Polak wiedział o tym, że taką rocznicę obchodzimy, wiedział o tym, że może w każdej chwili z tych bezcennych skarbów korzystać. I to nie tylko naukowcy, każdy z nas może sięgnąć po tę spuściznę dziejową, spuściznę tworzoną, można powiedzieć, w bardzo trudnych warunkach, o którą z całą pewnością my dzisiaj powinniśmy dbać, wyrażać uznanie, ale nie tylko, wyrażać także troskę i pomagać w dalszym wspaniałym rozwoju. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Na tym kończymy 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.